inspekcją sanitarną, lotniskiem, Urzędem Lotnictwa Cywilnego i wszystkimi innymi instytucjami dotyczących transportu osób z Chin. Również 25 stycznia nastąpiła koordynacja pomiędzy konsultantami w dziedzinie chorób zakaźnych oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie transportu trzech obywateli z Chin do Polski.

28 stycznia nastąpiło spotkanie robocze w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i rozesłanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia komunikatu dotyczącego zasad postępowania do wszystkich świadczeniodawców poprzez systemy elektroniczne SZOI i inne. Również został wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia obowiązek monitorowania i raportowania stanu łóżek zakaźnych. 28 stycznia, czyli tego samego dnia, kiedy rozsyłaliśmy komunikat dotyczący zasad postępowania, Hongkong i Mongolia wprowadzają częściowe zamknięcie granic z Chinami.

Przekazano do tych wszystkich instytucji opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego materiał o sposobie pobierania i przesyłania materiału od pacjenta do laboratorium PZH. Został opublikowany apel prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz głównego inspektora sanitarnego do środowiska medycznego z prośbą o przekazywanie wiarygodnych informacji oraz została przekazana do stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz do Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Lotnictwa Cywilnego aktualizacja zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem w podróży lotniczej. Dopiero 30 stycznia nastąpiło potwierdzenie transmisji z człowieka na człowieka - to był pierwszy przypadek w Stanach Zjednoczonych - i dopiero 30 stycznia WHO decyduje się na wprowadzenie stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym.

Przekazano ustalenia dotyczące bezpieczeństwa europejskiego.

2 lutego, czyli dzień później, zorganizowano ewakuację Polaków z obszarów zagrożonych z Chin. Na lotnisku wojskowym we Wrocławiu wylądowały dwa samoloty z 30 Polakami. 3 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zebrał się zespół roboczy do spraw sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem. oraz odbyło się spotkanie z ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w celu przekazania informacji dotyczącej sytuacji epidemiologicznej w Chinach. Jednocześnie raportowaliśmy do ECDC, jeśli chodzi o liczbę miejsc kwarantannowych, liczbę miejsc izolacyjnych oraz stan epidemiczny w Polsce.

7 lutego na posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego przedyskutowano sprawę ewakuacji pięciu osób z Chin, a 8 lutego przyjęto kolejne pięć osób z Chin na lotnisku w Warszawie.

Teraz następuje etap, w którym wirus dociera do Europy.

To oznacza, że pojawiły się ogniska zarażenia. 23 lutego włoska Rada Ministrów zatwierdziła dekret z mocą ustawy, który wprowadza środki dotyczące powstrzymania i zarządzania sytuacją. Następnego dnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkał się zespół roboczy do spraw sytuacji epidemiologicznej oraz odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Zdrowia z udziałem PLL LOT, Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie działań dotyczących również Polaków wracających z Włoch. 25 lutego zostało przesłane pismo do podmiotów leczniczych w sprawie możliwości wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie masek i kombinezonów z Agencji Rezerw Strategicznych. Jednocześnie wysłałem pismo do prezydencji Unii Europejskiej, do prezydencji chorwackiej w sprawie pilnego spotkania ministrów zdrowia w celu przedyskutowania sytuacji epidemicznej w Europie.

Jednocześnie został zatwierdzony krajowy plan działania na wypadek wystąpienia w Polsce przypadków podejrzenia lub zakażenia SARS-CoV-2.

27 lutego w rozporządzeniu ministra zdrowia nowy koronawirus został włączony do ustawy o chorobach zakaźnych, a jednocześnie przekazane zostały algorytmy postępowania - poprzez kanały NFZ oraz kanały inspekcji sanitarnej i współpracujących organizacji, takich jak choćby Porozumienie Zielonogórskie - do wszystkich POZ, AOS, czyli ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz do ratownictwa medycznego. Tego samego dnia, czyli 27 lutego, odbyło się spotkanie pana ministra Piontkowskiego z kuratorami i zostały przekazane wytyczne inspekcji sanitarnej dla szkół i dla rodziców. Tego samego dnia, czyli 27 lutego, wieczorem została podjęta decyzja przez wojewodę o odbywaniu się Intel Extreme Masters w Katowicach bez udziału publiczności. Jest to istotne o tyle, że Szwajcaria dwudziestego ósmego, czyli następnego dnia, wprowadziła ograniczenia dotyczące zgromadzeń masowych. Dwudziestego ósmego nastąpiło spotkanie pana premiera z wojewodami. Decyzją pana premiera zalecono wojewodom wprowadzenie stanu podwyższonej gotowości jednostek ochrony zdrowia zgodnie z art. 30 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zobligowano do zorganizowania całodobowego działania laboratoriów inspekcji sanitarnych, do bieżącej analizy przez inspekcję sanitarną i głównego inspektora sanitarnego ryzyk związanych z organizacją imprez masowych na terenie wszystkich województw oraz do wydawania zaleceń GIS-u wojewodom w sprawie imprez masowych. Jednocześnie zapadła decyzja premiera o uruchomieniu rezerwy budżetowej w wysokości 100 mln zł na najbliższe działania związane z przygotowywaniem się kraju do epidemii wirusa korona. Nastąpiło uruchomienie dodatkowych sześciu laboratoriów oraz dostarczenie do wszystkich tych laboratoriów testów na wirusa. Wcześniej mieliśmy aktywne dwa laboratoria. Wysłane zostały przez NFZ kolejne zalecenia i aktualizacja tych zaleceń do wszystkich podmiotów leczniczych. Przekazany został mój list do Sekretariatu Episkopatu Polski z prośbą o odczytanie go we wszystkich kościołach. Dwudziestego dziewiątego zostały dostarczone do wszystkich laboratoriów kolejne partie testów, a z Agencji Rezerw Materiałowych po analizie wniosków zostały rozwiezione przez Ministerstwo Obrony Narodowej środki do dziewięciu portów lotniczych oraz 30 szpitali, w których strukturach znajdują się oddziały zakaźne. W związku z różnymi doniesieniami 1 marca został powołany w Narodowym Funduszu Zdrowia zespół do monitorowania prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem przez podmioty lecznicze. Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia wydrukował i rozdystrybuował 100 tys. plakatów informacyjnych do świadczeniodawców i do aptek.

obecnie mamy 79 oddziałów, w których jest ponad 2900 łóżek zakaźnych. Każdy taki szpital zgodnie z dyspozycją wojewody ma opracowane plany zwiększenia liczby tych łóżek ponaddwukrotnie. W Ministerstwie Obrony Narodowej i podległych szpitalach jest kolejne blisko 80 łóżek szpitalnych i również istnieje możliwość zwiększenia tego stanu ponaddwukrotnie. Wszystkie szpitale otrzymały wytyczne, jak powinny postępować. Jest bieżące monitorowanie wojewodów dotyczące tego stanu. Została uruchomiona Agencja Rezerw Materiałowych. Środki ochrony osobistej zostały rozdysponowane do szpitali, które zgłaszały niedobory. Laboratoria mogą w tej chwili wykonywać - i mają maksymalną przepustowość - ponad 1200 testów na dobę.

Wojewodowie potwierdzili przygotowanie szpitali zakaźnych na wypadek pojawienia się ognisk zakażeń w Polsce.

Jednocześnie działania informacyjne obejmowały bardzo szerokie informowanie polskiego społeczeństwa. Szanowni Państwo! Oczywiście wirus pojawi się niedługo w Polsce, dlatego że wszystkie kraje WHO i eksperci mówią, że nie ma możliwości ograniczenia rozprzestrzeniania się tego typu wirusa o takiej zakaźności. Musimy być przygotowani na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Nasze działania, jak państwo słyszeliście, prowadzą do tego, żeby wszystkim przekazać informacje, jak postępować, dostarczyć brakujące środki i zapewnić informacje Polakom. W sytuacji epidemicznej, w sytuacji, w której następuje siłą rzeczy strach przed nowym, niezwykle istotne jest to, żeby trzymać się instrukcji. Poza tym jest to pierwsza epidemia w Polsce od czasu tak szerokiego dostępu do mediów społecznościowych. To jest też niezwykle ważne, dlatego że poprzez te media możemy dystrybuować informacje rzetelne i prawdziwe oraz informacje, które nie są sprawdzone. Tak jak państwa informowałem na wielu konferencjach prasowych i w publikacjach, monitorujemy w tej chwili na bieżąco sytuację wyników ze wszystkich laboratoriów w Polsce. Jeśli tylko pojawi się pozytywny wynik, jakikolwiek by to był pacjent, opinia publiczna zostanie o tym natychmiast poinformowana i państwo oczywiście również. To, że się pojawi, jest pewne. Zależy, jak na to zareagujemy i w jaki sposób będziemy informować pacjentów, co robić.

Dziękuję, panie ministrze.

Bardzo proszę.

Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zadaniem dzisiejszych obrad Wysokiej Izby jest, jak rozumiem, wypracowanie jak najlepszej strategii - strategii reakcji na epidemię, która dzisiaj zatrzęsła Chinami, zatrzęsła częścią Europy, i my w najlepszy możliwy sposób przygotowujemy się również na jej nadejście. Jesteśmy przekonani, że każda skuteczna i mądra strategia musi być poprzedzona dialogiem, musi być poprzedzona najlepszymi praktykami, które są wdrażane do systemu. My - jak przedstawił pan minister Szumowski - od samego początku, a nawet wyprzedzając większość krajów Unii Europejskiej. Również ta debata jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo poważnie traktujemy ten problem, i chciałem bardzo podziękować panu prezydentowi za zwołanie posiedzenia Wysokiej Izby, ponieważ będzie to dla nas. ponieważ będzie to dla nas dobra okazja do przedyskutowania aktualnego stanu sprawy.

Dlatego chroniąc zdrowie Polaków, zdecydowaliśmy się zainicjować szereg działań na forum Unii Europejskiej.

Również w zeszłym tygodniu rozmawiałem z premierem Andrejem Babišem i z premierem Viktorem Orbánem i zaproponowałem, żebyśmy w tym tygodniu spotkali się w ramach Grupy Wyszehradzkiej, aby przedyskutować kwestię koronawirusa. Dziś rano kontaktowałem się z premierem Andrejem Babišem i okazuje się, że w Czechach są trzy pierwsze zarejestrowane przypadki koronawirusa, więc rzeczywiście jest wysoce prawdopodobne, niemal pewne, że taki przypadek pojawi się i u nas.

To również z naszej inicjatywy nastąpiło przesunięcie 250 mln euro środków w budżecie Unii Europejskiej na walkę ze skutkami, na walkę z przyczynami koronawirusa, rozprzestrzeniającej się epidemii. Także w szczególności krajom południa Europy zależy na tym, żeby północna Europa, gdzie tych przypadków jest jeszcze cały czas dużo mniej, współpracowała z nimi w sposób jak najbardziej harmonijny, jak najbardziej zgodny, ponieważ południe Europy bardzo obawia się dalszego rozprzestrzeniania się wirusa po Europie. Dlatego razem z partnerami z Europy musimy zrobić wszystko, żeby uspokoić lęki, opanować sytuację, pomóc opanować sytuację, w szczególności naszym południowym sąsiadom, i żeby odbyło się to ponad granicami, ponad partyjnymi podziałami, a więc po prostu w dialogu i ponad bieżącymi różnicami zdań.

nie wykorzystywali jej w taki sposób również, który wzbudza niepokojące sygnały w całym społeczeństwie. Eksperci twierdzą, że dzisiaj mamy do czynienia z kilkoma ogniskami zakażania epidemią koronawirusa na całym świecie i dlatego podjęliśmy szczególne działania, jeśli chodzi o kraje, które już dzisiaj takie epicentrum epidemii stanowią, są to przede wszystkim Chiny, ale również Korea Południowa czy Włochy.

I również bardzo mocno proszę, żeby stosować się do tych reguł informowania wszystkich wracających podróżnych, proszę o wypełnianie wszystkich kwestionariuszy, ponieważ są one niezwykle ważne dla Głównej Inspekcji Sanitarnej, jeśli chodzi o rejestrowanie wszelkich możliwych ruchów potencjalnych pacjentów - pacjentów, obywateli, Polaków, którzy mogą być nosicielami tego typu wirusa.

21 stycznia generalny inspektor sanitarny opublikował odpowiednie komunikaty dla podróżujących. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy ze zdecydowaniem doprowadzili do ewakuacji Polaków przebywających w Chinach, na najbardziej zagrożonych terenach. W codziennym trybie spotyka się sztab zarządzania kryzysowego. Dokładne informacje przedstawiają na nim minister zdrowia, minister spraw wewnętrznych i administracji bądź jego przedstawiciele.

Wszyscy jesteśmy, szanowni państwo, na froncie walki, ale niech to będzie front walki z koronawirusem, a nie front walki politycznej. W tej walce wszyscy musimy być po jednej stronie. Apeluję o to, bardzo o to proszę. Aby powstrzymać koronawirusa, potrzebujemy nie tylko współpracy między resortami, potrzebujemy również współpracy pomiędzy rządem centralnym a samorządami, ale także między rządem a opozycją. Przypomnę, że kiedy wybuchło zagrożenie rosyjskie w 2014 r., wiosną 2014 r., ówczesny lider opozycji pan prezes Jarosław Kaczyński zaapelował o współpracę z rządem, aby ustabilizować sytuację, uspokoić sytuację, w odpowiedzialności za państwo i w poczuciu racji stanu. Dzisiaj wiemy, że lotniska to są takie okna na świat. Na lotniskach wprowadziliśmy bardzo szczegółowe procedury, również takie procedury, które są zupełnie niepotrzebnie czasami wyśmiewane. Faktycznie nie jesteśmy w stanie przecież zablokować granic, zamknąć granic przed koronawirusem, ale jesteśmy w stanie minimalizować jego dostęp na terytorium Polski. Dlatego jest mierzenie temperatury, dlatego ta kwarantanna, dlatego badanie już dzisiaj kilkuset osób od strony testów genetycznych, o czym mówił pan minister, po to, aby wykluczyć i natychmiast zlokalizować potencjalnie pojawiające się źródło tego typu zagrożenia. Agencja Rezerw Materiałowych dokonała dodatkowych zakupów, dodatkowych zamówień masek, maseczek i wszystkich tego typu sprzętów potrzebnych dla szpitali, potrzebnych dla służby zdrowia, po to, żeby w najbardziej odpowiedni sposób przygotować się do tej epidemii. Ten apel o odpowiedzialność i unikanie paniki jest bardzo ważny, ponieważ w przypadku wybuchu niepokojów, wybuchu paniki ci, którzy mogą najbardziej potrzebować pomocy medycznej, mogą mieć utrudniony do niej dostęp, dlatego że wiele osób, które takiej pomocy nie potrzebują, będzie akurat korzystało ze służby medycznej. Cały personel medyczny wie o tym doskonale, ale apeluję do Wysokiej Izby i za pośrednictwem Wysokiej Izby - bezpośrednio do wszystkich rodaków, aby takiej paniki unikać. Chciałbym zatem szczególnie mocno podkreślić konieczność zachowania pełnego profesjonalizmu oraz spokoju. W Internecie pojawiło się bardzo wiele nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji. To jest istotny czynnik ryzyka, którego nie powinniśmy lekceważyć, nie chcemy ignorować. Dlatego z tymi fake newsami z całą mocą walczy główny inspektor sanitarny i my również prezentujemy prawdziwe, rzetelne, wiarygodne informacje jako odpowiedź na te wszystkie fake newsy. Zresztą władze Stanów Zjednoczonych, mogę je niejako zacytować, przytoczyły przykłady różnych fejkowych kont na Twitterze, na Instagramie czy Facebooku, pochodzenia rosyjskiego, jak to zostało powiedziane. Różne trolle, różni pseudointernauci po prostu sieją niepokój, po prostu starają się zburzyć profesjonalne podejście do zaadresowania tego problemu. Wysoka Izbo! Uzasadniony niepokój Polaków łatwo jest spotęgować. Łatwo jest spotęgować pospiesznymi komentarzami. Łatwo jest spotęgować poprzez nieodpowiedzialne wpisy w Internecie. Wystrzegajmy się tego.

Potrzebne są w związku z tym współpraca i spokój. O to właśnie bardzo proszę. Nie ma co insynuować, że wirus pojawił się na terenie kraju, kiedy mówimy o tym od samego początku, że natychmiast, jak się wirus pojawi, o tym poinformujemy. Nie chciałbym, aby dziś Polska była najbardziej zagrożona epidemią nieodpowiedzialności, ponieważ taka epidemia nieodpowiedzialności może rzeczywiście doprowadzić do szerszego rozprzestrzeniania się wirusa, niż przeciwnym wypadku miałoby to miejsce. Takie spekulacje internetowe czy granie zdrowiem Polaków jako kartą polityczną jest niebezpieczne. Na to, szanowni państwo, nie ma oczywiście szczepionki. Na to nie ma mojej zgody. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak zaapelować do wszystkich polityków, w szczególności polityków opozycji, którzy uczestniczą czasami w tej grze, czasami są pewnie prowokowani przez różnych internautów, o powagę. Kluczowa jest profilaktyka. Tak, również ta profilaktyka, która brzmi tak prosto, banalnie: mycie rąk, dezynfekcja, po prostu higiena. Wszystkie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i agend specjalistycznych na to wskazują i o to również proszę, o to również apeluję.

Zanim zatem dojdzie do wybuchu epidemii koronawirusa, musimy skutecznie walczyć z epidemią dezinformacji. Przed nią przestrzega szef Światowej Organizacji Zdrowia. Szanowni Państwo! Jest to test odpowiedzialności, test zgody, test wspólnej, zgodnej walki z dezinformacją, fake newsami, trollami internetowymi, które wzbudzają tylko niepotrzebnie społeczny niepokój. Mam nadzieję, że zostanie wynaleziona, ale musimy i chcemy współpracować ze wszystkimi siłami politycznymi, ażeby to zagrożenie minimalizować, żeby walczyć wspólnie o zdrowie publiczne.

Weźmy sobie wszyscy do serca to zalecenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu premierowi. Sejm ustalił, że dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 15-minutowych oświadczeń w imieniu klubów oraz 7-minutowego oświadczenia w imieniu koła. Otwieram dyskusję.

Szanowny Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Panie Prezydencie! To była ważna inicjatywa i dziękuję za tę inicjatywę panu prezydentowi, tak jak dziękuję pani marszałek za zwołanie tego posiedzenia Sejmu.

Warto było wysłuchać stanowiska pana ministra, pana premiera. Dziękuję za przedstawienie tej rzetelnej informacji, tak jak dziękuje za tę ciężką pracę, która toczy się tak naprawdę od 2 miesięcy. Dziękuję za te działania, które państwo podjęliście, pomimo tego - co należy raz jeszcze podkreślić - że koronawirusa jeszcze w Polsce nie ma, choć, jak słusznie zauważył pan minister, jest to zapewne niestety tylko kwestia czasu. Są codzienne posiedzenia sztabu kryzysowego, są różne inne działania. Warto podkreślić, szanowni państwo, że chodzi tu o codzienną pracę inspekcji sanitarnej, 16 tys. pracowników, których często nie zauważamy, wielu laboratoriów, które jak słyszeliśmy, są czynne i aktywne 24 godziny na dobę, ale także o ciężką pracę wielu innych służb medycznych: lekarzy, pielęgniarek, innego personelu, którzy zostali poinstruowani i są gotowi, przygotowani na ewentualne działania związane z pojawieniem się epidemii w Polsce. W tym wszystkim oczywiście potrzebny jest spokój, potrzebna jest odpowiedzialność, potrzebne są profesjonalizm, powaga i ciężka praca. Powiedziałem przed chwilą o ciężkiej pracy, która jest wykonywana przez różne służby państwowe tak naprawdę codziennie, nieomal 24 godziny na dobę. Ale także, szanowni państwo, oprócz tej pracy, oprócz profesjonalizmu różnych służb i przygotowania tych służb, niezwykle ważna jest odpowiedzialność, którą wszyscy również wspólnie dźwigamy. To naprawdę niezwykle ważne. Szanowni Państwo! Myślę, że mogę się tu zwrócić do przedstawicieli różnych klubów.

Myślę, że wszyscy powinniśmy - i taką mam nadzieję - zdać egzamin z odpowiedzialności. My w Komisji Zdrowia zajęliśmy się problemem tej epidemii czy zagrożenia tą epidemią już 3 tygodnie temu. Wówczas dyskutowaliśmy, podkreślę, zgodnie, ponad podziałami, niezależnie od klubu, w pełnej zgodzie na temat tego, co można, co należy zrobić, i wysłuchaliśmy informacji zarówno ministra zdrowia, jak i głównego inspektora sanitarnego. W poczuciu tej odpowiedzialności, szanowni państwo, trwajmy dalej.

Dziękuję stronie opozycji za przygotowanie dwóch krótkich projektów. Odbieram to osobiście jako troskę o państwo, chodzi o to, że chcieliście państwo włączyć się w te działania związane z zagrożeniem epidemią. Ale przede wszystkim dziękuję rządowi za przygotowanie dużego dokumentu, dużej ustawy, która reguluje nie tylko kwestie związane

poszczególnych służb, uruchomienia środków finansowych, różnych zagrożeń, które dotyczą chociażby miejsc takich jak lotniska. Szanowni Państwo! Trzeba w tym miejscu także podziękować takim służbom jak wojsko. Jeśli chodzi o ewakuację Polaków z Chin to m.in. dzięki wojsku udało się to przeprowadzić bardzo sprawnie. To naprawdę jest przykład dobrego współdziałania różnych resortów w ramach jednego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo! Wreszcie odbywają się także narady i spotkania z kuratorami, następnie także z wojewodami. Naprawdę, już na szczeblu wojewódzkim, na szczeblu lokalnym wiemy, co należy robić. Wojewodowie otrzymali odpowiednie dyspozycje, wiedzą, jak mają postępować, zresztą mówili o tym zarówno pan premier, jak i pan minister. Jest podwyższona gotowość.

Te działania wojewodów są koordynowane również z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. A więc służby państwa są przygotowane. Szanowni Państwo! Mimo że nie ma koronawirusa w Polsce, jesteśmy przygotowani. Były różne inne sytuacje, kiedy doganialiśmy, kiedy byliśmy nieprzygotowani, ale później oczywiście nadrabialiśmy ten stracony czas. Tym razem jeszcze przed epidemią służby państwowe są przygotowane. Szanowni Państwo!

Również w obrębie środowisk medycznych jest taka zgoda.

To naprawdę ważne.

Chodzi o informacje związane z pewnym elementarnym przestrzeganiem higieny.

To kwestia przestrzegania higieny, to kwestia odpowiednich działań, nie tylko mycia rąk. Szanowni Państwo!

Pani będzie miała swoje wystąpienie klubowe, będzie pani mówiła to, co pani chce. Szanowni Państwo! Kończąc, bo jeszcze jeden z kolegów będzie wypowiadał się w imieniu klubu: pamiętajmy o tych wszystkich faktach. Pamiętajmy i dbajmy o własne bezpieczeństwo, zwłaszcza te osoby, które mają obniżoną odporność. Jestem, szanowni państwo, przekonany, że państwo zda egzamin. Mam nadzieję, że zdamy egzamin my wszyscy. Również pani, pani poseł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To są wystąpienia klubowe, będzie miał swój czas. Będą wystąpienia państwa klubu, będziecie mówili to, co przygotowaliście. Proszę nie przeszkadzać, bo to jest naprawdę notoryczne. Panie bez przerwy przeszkadzają. Od tego jest mównica, żeby wyjść tutaj i zabrać głos. Nawet teraz pani próbuje ze mną dyskutować. Bardzo proszę, pan poseł Czesław Hoc. Proszę. Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Panie Premierze! Panowie Ministrowie! Nawiązując do tak szczegółowych i profesjonalnych, spokojnych wystąpień pana premiera, pana ministra i pana przewodniczącego. oczywiście mogę zaapelować, byśmy w tej chwili zresetowali wszelkie polityczne emocje, wszelkie polityczne narracje, które nie służą sprawie. Myślę, że kilka słów powinno być dzisiaj bardzo wyraźnie wyartykułowanych, mianowicie: spokój, bezpieczeństwo, roztropność, zaufanie i pokora. Proszę państwa, do naszego domu wdziera się niebezpieczny intruz, koronawirus.

Wirus SARS, który wywoływał ostrą niewydolność oddechową - śmiertelność wynosiła 10%. Tak więc spokojnie i bez paniki. Co wiemy dzisiaj o chorobie COVID-19?

Przecież pan minister wyraźnie powiedział, że w chwili gdy dowiedziano się o wirusie na świecie, podjęto szczegółowe, pilne działania.

Wszyscy przyjeżdżający z zagranicy, nie tylko z Włoch i Chin, otrzymują SMS-ową informację.

Proszę państwa, to są działania konkretne, spokojne, ale bardzo zdecydowane.

Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To prawda, należy działać spokojnie, rozważnie, merytorycznie, ale trzeba mówić prawdę. Bardzo długo pan premier mówił na temat niesprawdzonych informacji w Internecie. Dlaczego rząd, korzystając ze swoich możliwości, nie wychodził i nie mówił: nie, to nie jest prawda, jesteśmy w takiej a takiej sytuacji, zostało przygotowane to i to.

Rząd powinien być przygotowany na wypadek sytuacji kryzysowych i na wypadek epidemii.

Nie może być tak, że pacjent, który idzie do lekarza na tym najniższym szczeblu, trafia na lekarza, który nie ma sprzętu, nie jest zabezpieczony przed tym wszystkim, nie ma maseczek, nie ma rękawiczek.

Mówi się o tym na lotniskach, wszystko świetnie funkcjonuje.

Coś nie działa, panie premierze, trzeba to sprawdzić. Oczywiście, że wszyscy ludzie racjonalnie myślący w takiej sprawie działają razem, wykonują zadania, które powinny być powierzone, ale trzeba ludziom mówić prawdę i pokazywać, co mają robić w takiej, a nie innej sytuacji. Kiedy w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na temat tej choroby i tego, że opozycja złożyła projekty ustaw, pani marszałek powiedziała, że to w ogóle nie jest potrzebne, rząd ma pewne możliwości, żeby w tej sprawie działać. Pan prezydent zaproponował zwołanie Sejmu, żeby wysłuchać informacji pana premiera, żebyśmy te informacje poznali, ale rano pan prezydent spotkał się z panem premierem, więc już te informacje miał. Albo traktujemy się poważnie, traktujemy się z zaufaniem i chcemy się szanować, albo robimy spektakle polityczne.

Jest system, służby pracują, ale chciałabym poznać plan dla zwykłych obywateli, jak mają się zachowywać.

Pani koleżanki apelowały o to, żeby nie było wycieczek poza temat koronawirusa, a jednak są. Bardzo proszę. Panie Premierze! Rzeczywiście chcemy rozmawiać, chcemy pomagać. Mam jeden bardzo prosty apel: czas wreszcie odrzucić tę butę i pogardę, które od ponad 4 lat macie wobec wszystkich, którzy mają inne zdanie lub są z innej części sceny politycznej.

Oczywiście z tą pogardą, z tą butą mówiliście, że nic takiego nie jest potrzebne, bo państwo działa świetnie. Rzeczywiście państwo działało świetnie, kiedy minister zdrowia z panem prezydentem jeździli na nartach, podczas gdy trzeba było zajmować się sprawami najważniejszymi.

Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby przyjąć konkretne rozwiązania. Dzisiaj jesteśmy tutaj, dlatego że przez ostatni czas po raz kolejny zamiast zajmować się istotnymi dla Polaków kwestiami, zajmowaliście się walkami wewnętrznymi, walkami gangów wewnątrz waszej koalicji, walkami w ramach służb specjalnych. Nie zajmowaliście się prawdziwymi, realnymi problemami. Dzisiaj jesteśmy tutaj, ponieważ nie potraficie korzystać z tych procedur, które od lat w Polsce obowiązują. Przecież od 2007 r. obowiązują jasne i czytelne przepisy, zresztą przygotowane przez wasz rząd, które potem przejęliśmy i wprowadziliśmy. Nie potraficie korzystać z tych procedur. Kiedy w zeszłym tygodniu prosiliśmy i apelowaliśmy: zróbmy specjalne posiedzenie Sejmu, przyjmijmy rozwiązania ustawowe, to przecież z ust pani marszałek, z ust waszych ministrów padały sformułowania, że nic się nie dzieje, że nie potrzebujemy żadnych nowych rozwiązań. Niestety nawet koronawirusa wpisujecie w kampanię wyborczą. To jest bardzo, bardzo nieodpowiedzialne i złe. Mam apel z tego miejsca do pana prezydenta. Panie prezydencie, pan ma w rękach olbrzymie narzędzie. Jak wiemy, dwukrotnie sąd zmusił pana premiera do tego, by odwoływać nieprawdę w pana słowach. I dzisiaj pan premier mówi o tym, żeby sprawdzić, żeby walczyć z fake newsami. Panie prezydencie, to jest test dla pana. W pana rękach leży rozwiązanie, w przypadku którego 2 mld zł polskich podatników mogą iść na poprawę ochrony zdrowia Polek i Polaków, mogą iść na służbę zdrowia, mogą iść m.in. na zwiększenie liczby etatów specjalistów, na zwiększenie nakładów w służbie zdrowia, zwiększenie oddziałów zakaźnych, na poprawę bezpieczeństwa Polek i Polaków, a nie na produkcję fake newsów w tzw. publicznych mediach. To jest ten test, panie prezydencie. Dzisiaj ta debata jest rzeczywiście o tym, jak wspólnie możemy rozwiązywać problemy, które stoją przed naszą wspólną ojczyzną, ale żeby to zrobić, trzeba nie tylko mówić okrągłe słowa, które padają z ust pana premiera, ale trzeba konkretnych czynów. I dzisiaj mówimy wyraźnie: tak, jesteśmy tutaj po to, żeby wypracować odpowiednie rozwiązania, ale jesteśmy też po to, żebyście państwo odpowiedzieli, dlaczego do tej pory nie działaliście, dlaczego do tej pory wybieraliście narty zamiast sztabów kryzysowych, [[Oklaski]] dlaczego do tej pory nie przeznaczyliście większych środków, większej pomocy finansowej na służbę zdrowia, tylko z roku na rok zwiększacie wydatki na propagandę. Panie Prezydencie! Czas na realizację waszych obietnic. Czas na to, by Polacy przekonali się, czy chcecie wspólnie z opozycją jednym głosem załatwić najważniejsze problemy dotyczące tego, co przed nami, czy tylko i wyłącznie udajecie. Mam wielki apel, by nie wykorzystywać spraw, które powinny być ponad wszelkimi podziałami, by nie wpisywać ich w kalendarz wyborczy. Jeszcze w zeszłym tygodniu broniliście się przed debatą w Senacie i informacją rządu na temat sytuacji związanej z koronawirusem. Po co to wszystko? A potem. Co się zmieniło od tego czasu? Czy to, że chcieliście to wpisać. Bardzo dobrze. Znaczy, świetnie, że to mówicie, ale źle, że tak się dzieje. Chcieliście to wpisać w kampanię wyborczą? Panie prezydencie, pan ma dużo lepsze narzędzia. 2 mld zł dla polskiej służby zdrowia zamiast dla produkcji fake newsów, zamiast dla przemysłu pogardy. Zamiast dzielenia Polaków może pan zrobić coś bardzo, bardzo dobrego. Szanowni Państwo! Panie premierze, pan skupiał się na Internecie. Wiem, że być może w waszych szeregach są tacy eksperci, nie wątpię, którzy znają się właśnie na manipulacjach w Internecie, ale panie premierze, to nie osoby ze Wschodu, to nie trolle, to polska kobieta, to pacjentka jednego ze szpitali obnażyła prawdę o waszej nieudolności. To pani Ania z Krotoszyna pokazała, jak państwo nie działa. I dzisiaj przyznał to nawet sam minister zdrowia, mówiąc. Zabrakło słowa: przepraszam. Ja z tego miejsca chcę zadeklarować, że jesteśmy gotowi do każdej merytorycznej pracy. Jesteśmy gotowi do tego, by w sprawach wagi państwowej być na każde zawołanie i pracować w tej Izbie. Tylko że na razie to wy zorganizowaliście pracę w tej Izbie w ten sposób, że mamy po jednym posiedzeniu na miesiąc. To wy zorganizowaliście tak pracę, żeby Sejm się nie zbierał. I teraz oczywiście udajecie, że chcecie coś naprawiać. Ale gdzie byliście przez ten czas? Gdzie był minister zdrowia? Pan nawet podobno we Włoszech na nartach był. Dwa razy w Polsce, to rozumiem. Ale jeszcze do Włoch pan pojechał? Znaczy, na Boga, są pewne granice hipokryzji i są pewne granice tego, jak państwo powinno działać. I dzisiaj to jest prawdziwy test, ale to jest test, który musi zdać większość parlamentarna. My jako opozycja jesteśmy gotowi, raz jeszcze podkreślam, do merytorycznej pracy. Tylko jak ta praca z waszej strony wygląda? W zeszłym tygodniu słyszymy: niepotrzebna ustawa. Zbieracie na gwałt Komisję Zdrowia. W tym projekcie znajdują się rozwiązania co najmniej kuriozalne, a w części bardzo kontrowersyjne. To jest ustawa, która powinna być procedowana w zwykłym trybie. Ja mam wielkie obawy, czy po raz kolejny nie wykorzystujecie sytuacji do tego, by wprowadzić procedury, które z normalnymi zasadami dobrze funkcjonującego, bezpiecznego, sprawnego państwa nie mają absolutnie nic wspólnego.

I dzisiaj to jest elementarny test nie tylko na sprawność państwa, bo ten test już niestety oblaliście, ale to jest test na elementarną przyzwoitość, przyzwoitość, czy chcecie państwo, żeby wspólnie, w sprawach kluczowych, nie było podziałów politycznych, czy chcecie po raz kolejny dzielić Polaków, czy chcecie po raz kolejny dzielić Izbę. Mówimy wyraźnie: chcemy pracować. Ale dzisiaj piłka jest po waszej stronie. Dziś test na przyzwoitość musi zdać prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w którego rękach leżą środki finansowe, które mogą być przeznaczone na naprawdę najważniejsze potrzeby Polek i Polaków, m.in. na ochronę i na służbę zdrowia. I dzisiaj, i tu się zgadzam, panie premierze, jest też test na to, czy wybierzecie politykę fake newsów i manipulacji i przeznaczycie 2 mld zł na tzw. publiczną telewizję, czy wspólnie przeznaczymy 2 mld zł na to, by rzeczywiście polski system ochrony zdrowia działał lepiej, skuteczniej, działał w sposób profesjonalny i żebyśmy my wszyscy, wychodząc dzisiaj z tej sali, mogli powiedzieć: tak, udało nam się wspólnie wypracować to, czego oczekują Polki i Polacy. Zapraszam, pani poseł Marcelina Zawisza, Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Szanowna Wysoka Izbo! Chciałabym zacząć od tego, że chciałabym przywitać kandydata Lewicy na prezydenta Roberta Biedronia. Pani poseł, proszę się nie zapominać. Dopiero wczoraj w nocy pojawił się rządowy projekt. Ale mam również pytania do dzisiejszych wystąpień. Ani w projekcie, ani w dzisiejszych wypowiedziach nie widzą państwo w ogóle problemu 45% pracowników, którzy chorzy chodzą do pracy, bo boją się jej utraty. Nie widzę zwiększenia budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, której inspektorzy mogliby wspierać pracowników i kontrolować, czy w tak kluczowym momencie przestrzegane jest prawo pracy. Projekt pomija też osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Powinni mieć możliwość pracy zdalnej, ale jak zwykle. dla polskiego państwa są niewidzialni. Brak środków na akcje informacyjne dla Państwowej Inspekcji Pracy. Polki i Polacy nadal nie wiedzą, jakie mają prawa. Nie wiedzą, że w sytuacji, gdy zostaną skierowani na przymusową kwarantannę, mają prawo do zwolnienia chorobowego, że gdy zachoruje ich dziecko, mają prawo do urlopu na to dziecko. Ale brak wiedzy to tylko jeden z aspektów. Nie ma świadczeń dla osób nieubezpieczonych. Koronawirus nie będzie wybierał tych, którzy płacą składki. Nie rozumiem, dlaczego rząd w tak kluczowej sprawie stosuje neoliberalne rozróżnienie na ubezpieczonych i nieubezpieczonych. Wszyscy jesteśmy obywatelami tego kraju. I nasz rząd powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby nas przed tym zagrożeniem uchronić. Nie widzę zwiększenia budżetu inspekcji sanitarnej, która będzie odgrywała kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa. Są środki na konkretne działania. Nie ma pieniędzy na nadgodziny, na dotrudnienie. Znowu zakładacie, że ludzie będą harować za grosze. I co najważniejsze, zupełnie nie słyszę informacji na temat tego, czy rząd zadba o bezpieczeństwo lekowe Polski. Obecnie duża część substancji czynnych, z których tworzy się leki, produkowana jest w Chinach. Czy Polsce grozi brak leków? Jeżeli tak, to których? Jak rząd planuje zaadresować ten problem w przyszłości? Czy zabezpieczone 40 mln wystarczy na obsługę administracji oraz produkcję leków, gdy zabraknie dostaw z Chin? O reszcie wątpliwości opowiedzą moi koledzy i koleżanki. Proszę bardzo, pan poseł Marek Rutka, Lewica. Panie Prezydencie! Wysoka Izbo! Lewicowy Kandydacie na Prezydenta! Od samego początku Lewica nawołuje do zachowania spokoju, kierowania się zdrowym rozsądkiem i niewykorzystywaniem tej sytuacji do bieżących rozgrywek politycznych, a tym bardziej w toku kampanii wyborczej. Z drugiej jednak strony odnosząc się do sokratejskiego rozumienia polityki jako roztropnej realizacji wspólnego dobra, nie możemy jako poważna siła polityczna, na którą głos oddało ponad 2 mln obywateli i obywatelek, pozostawać obojętni wobec tego, jak w obliczu poważnego zagrożenia postępuje obecna władza. Pan premier, minister zdrowia, minister spraw wewnętrznych i administracji zwołali konferencję prasową poświęconą zagrożeniu koronawirusem COVID-19 w poniedziałek, 24 lutego, podczas gdy trzy pierwsze potwierdzone przypadki koronawirusa COVID-19 ogłoszono w północnych Włoszech już w piątek, 21 lutego. Rząd potrzebował ponad 48 godzin na to, aby zwołać konferencję prasową, powiedzieć, że będą rozsyłane SMS-y z informacjami dla powracających z zagranicy o tym, jak trzeba postępować w sytuacji zagrożenia, że nasze służby są w pełnej gotowości. O ile jednak rząd potrzebował weekendu na reakcję, to wirus na pewno w tym czasie wolnego nie miał. Jest wielce prawdopodobne, że dotarł do Polski wraz z powracającymi z północnych Włoch rodzinami, spędzającymi ferie w tamtejszych rejonach. Weekend 22–23 lutego był przecież ostatnim z tegorocznych ferii zimowych i - co istotne - dla dzieci z czterech województw, w tym największych: mazowieckiego czy dolnośląskiego. Mediana inkubacji wirusa według badań prowadzonych w Wuhanie wynosi od 3 do 24 dni. Tego samego zdania jest także odkrywca SARS. Strona rządowa apeluje o poważne podejście do problemu. Jak to się jednak ma do tego, że członkowie Komisji Zdrowia, a jestem jednym z nich, otrzymali SMS-a informującego o pilnym posiedzeniu komisji wczoraj o godz. 22.09, a kolejnego informującego, że druk znajduje się na stronie Sejmu - o godz. 23.23? Sama komisja została zwołana na godz. 8.45. Nie mamy do czynienia z niespodziewaną powodzią, trzęsieniem ziemi czy przypadkiem tsunami na Bałtyku, które wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin. O tym, że koronawirus dotrze do Polski, wiadomo od kilku dni, a nie od kilku godzin. Przedłożony projekt ustawy liczy 23 strony i zawiera szereg odniesień do innych aktów prawnych i w ciągu kilku nocnych godzin nie ma możliwości dokładnego zapoznania się z zawiłościami przedłożonej ustawy. Przedłożony projekt ustawy musiał być przygotowywany od kilku dni, a nie od wczoraj niedzielnego popołudnia. Dziś rano zadałem na posiedzeniu Komisji Zdrowia pytanie, od kiedy ministerstwo pracowało nad tym projektem, i nie dostałem na to pytanie żadnej odpowiedzi. Wspólnie z grupą posłów Lewicy 25 stycznia złożyłem interpelację nr 1675 w sprawie ryzyka szerzenia się na terytorium Polski epidemii koronawirusa. Do dziś, a minęło 37 dni, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Proszę, pani poseł Katarzyna Kotula, Lewica. Dzień dobry. Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Premierze! Lewica daleka jest od podsycania paniki i podgrzewania emocji i chcemy, żeby rząd działał w tej sprawie sprawnie, zapewniając bezpieczeństwo zdrowia i życia Polaków i Polek. Chcemy mieć też świadomość, że rząd zrobił dotychczas wszystko, aby faktycznie zapobiec temu, co przed chwilą minister nazwał epidemią strachu i paniki. Wiemy, co rząd proponuje w obecnej ustawie, ale chcemy zapytać też, co zrobiono dotychczas, a może chcemy zapytać po prostu też o to, dlaczego wystąpiły jednak pewne zaniechania.

Czy procedury te ulegną zmianie? Prosimy o informację, ile dotychczas zostało przeprowadzonych testów.

Jak to możliwe, skoro mamy 11 laboratoriów w trybie całodobowym i 1200 testów na dobę? Rozumiemy, że to od dziś. Wydaje się, że istnieje też konieczność publicznego raportowania przez głównego inspektora sanitarnego o ilości przeprowadzonych badań, liczbie osób, których to dotyczyło, i wynikach tych badań, tak jak się to robi w większości państw Europy. Dostęp do tych informacji to jedno z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Ponieważ tylko i wyłącznie dostęp do informacji może zagwarantować spokój w obliczu epidemii, zasadne wydaje się uruchomienie infolinii.

Mogą oni udzielić odpowiedzi, uspokoić albo zdecydować o wysłaniu karetki do zgłaszającego. Dlaczego uważam, że miejscem pozyskiwania informacji nie powinny być stacje sanitarno-epidemiologiczne, gdzie w przeważającej większości pracują osoby bez wykształcenia medycznego?

Pan poseł Zdzisław Wolski, Lewica. Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ustaliliśmy w klubie, że odniosę się konkretnie do szpitali jako bardzo ważnych podmiotów leczniczych, gdy mówimy o zwalczaniu koronawirusa. Moim zdaniem to dobrze, że rząd pracuje, wydaje instrukcje, jakieś wytyczne, zalecenia, ale tak naprawdę to nie rząd powinien być przygotowany, a same szpitale.

Wiemy, jak zaniedbany jest pion lecznictwa, jeżeli chodzi o choroby zakaźne. Do liczb, które podawali pan premier i minister zdrowia, nie będę się odnosił.

Brakuje specjalistów, brakuje pielęgniarek. Przypominam, że Lewica zawsze była przeciwko prywatyzacji szpitali.

Obserwuję to również z pozycji lekarza z 40-letnim stażem pracy. To w nich nadzieja. Natomiast odniosę się bardzo krótko do fatalnej rzeczy.

To przecież nie rząd zawinił, tylko lekarz, szpital.

Jeżeli tak mają być traktowani lekarze, pielęgniarki, ratownicy i inny personel, to naprawdę źle to. Apeluję, żeby tego nie robić. Jeszcze - już kończę - czy mamy regulacje? Jak on ma działać?

Pan poseł Wiesław Szczepański, Lewica. Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Czy moglibyśmy wiedzieć, jakie są ich wyniki? Które województwo z tym zalega, a które jest dobrze przygotowane? Jak wygląda współpraca wojewodów z samorządami? Niektóre narzekają na przepływ informacji. Podobno wojewodowie zaktualizowali wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego - plany, które zostały negatywnie ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przedmiotem kontroli była wówczas ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Według tego raportu w Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Cały czas utrzymywany jest dualizm rozwiązań prawnych, tj. funkcjonują struktury w ramach zarządzania kryzysowego i niezależnie od tego utrzymywane są formacje obrony cywilnej.

że brak przygotowania odpowiednich planów i procedur może po prostu jednak nie uskutecznić.

Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Możemy się różnić, możemy się spierać, ale w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w obliczu masy pytań i lęków, które są wśród naszych obywateli.

1577 osób zarażonych i 34 osoby, które zmarły. Śmiertelność jest wysoka.

A więc jest coś nowego, coś nieznanego, trzeba interweniować. Farmaceuci nie byli zaangażowani. Nie ma żadnej komunikacji z samorządem w Polsce. Dobrze, że zaprosiliście kuratorów, ale za organizację oświaty w gminie, w powiecie, w województwie odpowiadają samorządowcy. Nie dostali oni informacji, nie ma z nimi współpracy, nie ma rozmowy, nie ma przekazywania ulotek. 2 mln pacjentów codziennie korzysta z aptek, przychodzi, kupuje leki. Dobrze, że dzisiaj słyszymy o plakatach. Tylko czy te wszystkie działania nie są zbyt późne? Ja się nie dziwię, że one są spóźnione, ponieważ kiedy usłyszeliśmy o wystąpieniu choroby w Chinach, to w pierwszych doniesieniach, w pierwszych dniach minister zdrowia z głównym inspektorem sanitarnym nie mogli uzgodnić zdania.

Jeżeli główny inspektor sanitarny z ministrem zdrowia nie mają wspólnego zdania w pierwszych dniach wystąpienia wirusa, to jak polscy obywatele mają czuć się bezpiecznie? Kolejna sprawa. Co z oddziałami zakaźnymi? Panie ministrze, panie premierze, proszę o informację: Ile oddziałów zakaźnych zostało zlikwidowanych w ostatnich latach? Bo słyszymy, że dzisiaj jest gotowych do pracy 79 oddziałów, które mają ok. 2 tys. łóżek szpitalnych, mogą to zwiększyć. Dobrze. Ile było, jak przejmowaliście władzę? Czy nie było 119 oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych? Dlaczego ich liczba tylko do końca 2018 r. - bo takie dane opublikowaliście - spadła o 200 osób?

Nawet z tego tysiąca 30% jest w wieku emerytalnym. To pokazuje skalę zaniedbań, niedofinansowania oddziałów chorób zakaźnych w ostatnich latach.

Dobrze, że jest dzisiaj i się przysłuchuje tej debacie, ale kilka lat temu Paweł Kukiz na spotkaniu w innej sprawie zaproponował reformę ochrony zdrowia, żeby było mniej biurokracji, żeby pan prezydent stanął na czele. Nie zrobił tego. Nie zrobił tego przez 5 lat. Dobrze, że dzisiaj może wysłuchać tej debaty.

Mówicie o ankietach, które są wypełniane na pokładach samolotów.

To są pytania, panie ministrze. Naprawdę... wy uważacie, że jak wam ktoś wypowie wady, błędy, to jest to atak na was. To nie jest atak, tylko wskazanie, gdzie jest dzisiaj problem. Odzywał się pan minister infrastruktury. To czemu kierowcy tirów nie mieli informacji, gdy dojechali do północnych Włoch, jak się należy zachowywać? Czemu kierowcy autobusów nie mieli takiej informacji? Jak przemieszczają się Polacy pomiędzy Polską a Włochami najczęściej? Czy transportem samolotowym? Przejeżdżają samochodami i autokarami. Jeżeli idą na SOR w szpitalu, często w szpitalu wojewódzkim, to ten SOR - jeżeli dochodzi już do podejrzenia, to jest z ostatnich godzin informacja z Tarnowa - jest wyłączony. Kolejki wtedy do innych specjalistów, w innych przypadkach, wydłużają się do kilkunastu godzin. Czy 1200 testów dziennie wystarczy? Kolejna sprawa - oddziaływanie tej epidemii na gospodarkę. O tym nie było dzisiaj mowy. Rozumiem, że nie mówił o tym pan minister zdrowia, ale nie powiedział też o tym pan premier. Jaka będzie sytuacja z produkcją wielu komponentów, wielu substancji, które są wytwarzane w Chinach, a polskie firmy z tego korzystają? Czy jest jakikolwiek dialog prowadzony w tym zakresie, tak żeby przygotować polską gospodarkę? Padło już pytanie, ale ja je doprecyzuję.

My jesteśmy państwem, zresztą jak wiele niestety państw w Europie, uzależnionym od produkcji leków w Chinach. To nie dotyczy tylko i wyłącznie przemysłu farmaceutycznego, ale również przemysłu chemicznego i innych spraw związanych z gospodarką. Szanowni państwo, bądźmy zjednoczeni w walce o zdrowie Polaków nie tylko w momencie, kiedy przychodzi wirus, ale i wtedy, kiedy jest sprawa reformy ochrony zdrowia. Ona jest konieczna. Bez tego nie będzie bezpieczeństwa zdrowotnego Polski i Polaków. Nowa ustawa na koniec. Dobrze, że jest, tyle że ona nie jest rozwiązaniem systemowym. Ona jest daniem kompetencji, bardzo osobowych, wojewodom. Może jest taka dzisiaj potrzeba. Będziecie, rozumiem, to wyjaśniać.

To chyba jest słabe źródło finansowania.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Klimczak, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15.

Natomiast dzisiaj oczekiwałem, że będzie więcej mówione na temat pieniędzy, będzie więcej mówione na temat wsparcia sanepidu, będzie więcej mówione na temat zmian dotyczących oddziałów zakaźnych i ich finansowania, ponieważ dzisiaj widzimy, jaki problem mają te oddziały zakaźne, które przyjmują osoby, które już są podejrzewane o koronawirusa.

Dziękuję. Szanowni Państwo! W pierwszej kolejności chciałbym wyrazić swoje zdumienie, że posiedzenie Sejmu zostało zwołane na wniosek pana prezydenta i pan prezydent nie zdecydował się zabrać głosu. Jeżeli to posiedzenie Sejmu było uzasadnione z perspektywy Kancelarii Prezydenta i z perspektywy głowy państwa, to chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokładnie cele miał pan prezydent, zapraszając tutaj 460 posłów i uważając, że rząd czy Komisja Zdrowia pracują w sposób niewystarczający i że te głosy, które tutaj z mównicy sejmowej wybrzmiewają przez ostatnie 2 godziny, wnoszą coś więcej do naszej publicznej wiedzy na temat stanu przygotowań naszego państwa. Pozwolę sobie przypomnieć, że apelowałem w zeszłym tygodniu o zwołanie Rady Gabinetowej, na posiedzeniu której pan prezydent z pomocą również swoich doradców, bez udziału kamer, bez tych wszystkich spojrzeń posłów opozycji, mógłby zadać pytania członkom rządu o stan przygotowania naszego państwa na tę właśnie epidemię i oczekiwać szczerych odpowiedzi.

Jeśli posłowie opozycji mają informacje, że rząd coś ukrywa, to niech ujawnią fakty. Jeżeli natomiast nie macie państwo wiedzy o żadnych faktach, to proszę nie chwiać nastrojami społecznymi, [[Oklaski]] tylko spróbować robić to, co robi Konfederacja. Spróbujcie państwo choć przez to jedno nadzwyczajne posiedzenie Sejmu być opozycją merytoryczną. Zapewniam państwa. Panie Premierze! Panie Ministrze! Zadałem w zeszłym tygodniu cztery pytania w swojej interpelacji. Chciałbym poprosić o to, żeby zrobić pewien wyjątek od tego trybu ustawowego, iż posłowie czekają ok. miesiąca na odpowiedzi. Chciałbym poprosić o odpowiedzi w sprawie stanu przygotowania naszego państwa, zapasu odpowiednich materiałów i instrukcji pisemnych, które powinny być już we wszystkich placówkach ochrony zdrowia. Chciałbym poprosić o te odpowiedzi już dziś. Będę bardzo wdzięczny również panu prezydentowi za ujawnienie swoich wątpliwości, jeżeli takie ma, w kwestii stanu przygotowania naszego państwa i troski obywateli, którą wszyscy tu, w tej Izbie, jak sądzę, wspólnie w takiej groźnej sytuacji powinniśmy wyrażać. Panie pośle, każdy poseł, każdy polityk ma prawo zadawać rządowi pytanie, kiedy w sieci krążą właśnie sprzeczne informacje. Wysoka Izbo!

Ale jakie prawo wy, posłowie, macie, żeby szerzyć panikę wśród ludzi? straszycie ludzi. Od tego mamy ministra zdrowia, w normalnym kraju sprawę załatwia minister zdrowia. Co ma zrobić Sejm, panie prezydencie? W normalnym kraju minister zdrowia wstawia sobie tego koronawirusa na listę chorób zakaźnych i operuje na podstawie ustawy o chorobach zakaźnych. Nie trzeba żadnej specustawy na ten temat, po prostu i zwyczajnie. Proszę państwa, żyjemy w czasach, kiedy zwołuje się Sejm, żeby była demagogia, żeby się lały potoki słów. Nie, proszę państwa, potrzebujemy czynów, a nie słów. Bardzo proszę, pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Pani Marszałek! Panie Prezydencie! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Koronawirus to temat, który powinien być ponad podziałami politycznymi. To temat, który nie powinien być rozgrywany politycznie przez poszczególnych działaczy, kandydatów na scenie publicznej. To temat, który przynależy do sfery bezpieczeństwa państwa i w którym państwo powinno zdecydowanie zadziałać. Państwo powinno działać nie dziś, nie w zeszłym tygodniu, nawet nie w połowie lutego, bo pierwsze przypadki koronawirusa na naszym kontynencie były już miesiąc temu. To państwo, które dzisiaj reaguje nadmiernie, dlatego że w odpowiednim momencie nie zadziałało jak trzeba.

Bo gdyby tak było, to dzisiaj oprócz pana ministra zdrowia przemawiałby również pan minister Kamiński. Bo koronawirus, epidemia, czy w ogóle jakiekolwiek zagrożenie, które wkracza do państwa, uświadamia nam, że ta utopia, utopia świata bez granic, utopia, która miała być rzekomo zrealizowana po wejściu do Unii i NATO, nie istnieje. Że w momencie, kiedy państwo jest zagrożone, to służby specjalne, służby mundurowe tego właśnie państwa są ostatecznie odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli. Masowe powroty z ferii, również znacznej części lekarzy. Sytuacja w służbie zdrowia i tak jest bardzo zła. Dlaczego ministrowie finansów, resortów gospodarczych dzisiaj nie przemawiają? Przecież Chiny, fabryka świata we współczesnym podziale pracy, dzisiaj dostała zadyszki ze względu na tę epidemię, ta fabryka świata. To wszystko będzie miało wpływ, i ma już dzisiaj wpływ, na naszą giełdę, na funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw, również na nasz przemysł farmaceutyczny i na to, czy w Polsce są dostępne leki. Nie mamy dzisiaj kompleksowej informacji w tych sprawach. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania?

Pan poseł Rajmund Miller, Koalicja Obywatelska. Jest, dobrze. Był pan za drzwiami. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja mam jedno pytanie.

Czy jest pełne współdziałanie z państwami Unii Europejskiej? Nie da się postawić muru, płotu, jakichś różnych łapaczy, które tego wirusa gdzieś od nas odizolują. Jakie są polskie inicjatywy w Komisji Europejskiej, która działa poza posiedzeniami parlamentu, żeby aprobować (Dzwonek), wystawiać, dawać określone wskazówki, jak postępować w krajach członkowskich? Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Rajmund Miller, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Prezydencie! Wysoka Izbo!

Na tym posiedzeniu Komisji Zdrowia zwróciliśmy uwagę przedstawicieli ministerstwa na niezapisanie koronawirusa w ustawie o chorobach zakaźnych, co powodowało, że w sytuacjach, kiedy pacjent powinien być przymuszony, chory lub podejrzany o zachorowanie, dla zabezpieczenia zdrowia publicznego, do odbycia leczenia lub kwarantanny.

Przez te 2 tygodnie miało miejsce narażanie zdrowia publicznego w Polsce, bo ludzie chorzy i zarażeni mogli poruszać się wśród ludzi zdrowych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie!

Jak wygląda obecnie ścieżka przekazywania pacjentów z podejrzeniem koronawirusa do szpitali specjalistycznych? Czy szpitale specjalistyczne i oddziały chorób zakaźnych są przygotowane na dzień dzisiejszy na dezynfekcję pomieszczeń?

Ile jest takich sal w Polsce?

To ma być dopłata. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Protasiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Dziękuję, pani marszałek. Panie Premierze! Usłyszeliśmy tutaj gorące zapewnienia o wręcz międzynarodowej skali działań rządu zabezpieczających Polskę i Polaków przed negatywnymi skutkami działania koronawirusa. Ja będę mówił zatem o szczegółach bardziej przyziemnych.

który chce pójść zaniepokojony sytuacją i słuchający głównego inspektora sanitarnego kraju. I wreszcie czy maseczki również są dostępne? Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale oczekuję. Ona brzmi: nie. Ale być może od pana ministra bądź od pana premiera usłyszymy inną. Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Izbo! Standardem na lotniskach, np. w Japonii, są kamery termowizyjne. W ten sposób można już w pierwszym rzucie ocenić, czy ktoś może być podejrzewany o to, że jest zarażony lub w tym momencie jest w złym stanie zdrowia.

Bardzo proszę. Panie Prezydencie! Wysoka Izbo! Chciałbym skierować moje pytania do pana ministra Szumowskiego i zapytać o to, jak pan ocenia, panie ministrze, stan polskich szpitali w zakresie chorób zakaźnych. Pan premier podawał dzisiaj statystyki. I czy nie uważa pan, że rzeczywiście wieloletnie zaniechania w zakresie kontraktowania usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia spowodowały, że dzisiaj tak naprawdę jest ogromny deficyt? Drugie moje pytanie dotyczy szpitalnych oddziałów ratunkowych. Czy nie uważa pan, że decyzje, które podejmował pana poprzednik, były bardzo złe? Bo dzisiaj SOR-y są naprawdę najbardziej niebezpiecznymi miejscami. I czy przewiduje pan w tej chwili także pewną reorganizację, aby - jak mi tutaj kolega poseł podpowiedział - doprowadzić do takiej wstępnej segregacji, przepraszam, selekcji pacjentów, szczególnie tych chorych na choroby zakaźne? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Prezydencie! Tymczasem opozycja zadaje pytanie, po co ta dzisiejsza debata. Oto rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec na Twitterze w trakcie naszej debaty napisał: W tym czasie nosiciele koronawirusa zarażają setki kolejnych osób. To jest odpowiedzialne? To jest prawda? Dzisiaj pan minister, pan premier ujawnili całą prawdę.

Pani Marszałek! Panie Premierze! Koronawirus i ta epidemia, która się rozszerza po świecie, to nie jest wyłącznie choroba ludzi. To jest także choroba państw. Te, które są mało odporne, będą miały wielkie kłopoty. Te, które są odporne, sobie poradzą. Istotą tej odporności państw jest zaufanie obywateli do władzy publicznej. Poczucie, że władza publiczna wie, co robi, i wie, co mówi. Panie Premierze! Mianowany przez pana urzędnik, czyli pan Jarosław Pinkas, szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w zeszłym tygodniu, ba - w piątek, udzielił wywiadu, w którym powiedział, że właściwie nie wiemy, ile jest maseczek, że nie dla wszystkich starczy, a jeśli ktoś ma kłopoty z nimi, to niech sobie je zrobi z biustonoszy. To jest komunikacja władzy publicznej, która ma uspokoić tak naprawdę opinię publiczną? To jest ta odporność państwa, która ma spowodować, że mamy czuć się spokojni?

To nie jest prawidłowa komunikacja z opinią publiczną. Dziękuję, panie pośle. Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Panie Premierze! Rzeczywiście dzisiaj zajmujemy się specustawą.

Natomiast pewnie w sytuacji kryzysowej - gdyby ta ustawa już kilka lat temu była przyjęta - nie musielibyśmy dzisiaj przyjmować tej specustawy.

Bardzo proszę, pan poseł Marek Hok, Koalicja Obywatelska. Panie Prezydencie! Krótkie pytanie, panie ministrze. Dlaczego mamy tylko dwa ośrodki, właśnie dwa laboratoria diagnostyczne, i obydwa w tym momencie w Warszawie? Mówił pan minister, że jest sześć dodatkowych. W których miejscowościach one są? Dlaczego w każdym województwie, w każdym z 16 miast wojewódzkich takie laboratorium nie może funkcjonować? Czy te laboratoria są wyposażone w odczynniki, które są niezbędne do badań wirusologicznych?

W końcu: dlaczego tak długo? Czas oczekiwania: 72 godziny. Słynny przypadek z Krotoszyna - 88 godzin czekała pacjentka. Badania we Włoszech, badania w Niemczech trwają 8 godzin.

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Premierze! Wysoka Izbo! Usłyszeliśmy dziś od pana ministra zdrowia bardzo precyzyjną informację o podjętych działaniach przez polski rząd. I to już od pierwszych chwil, gdy komunikaty o koronawirusie pojawiły się w przestrzeni medialnej. Otrzymaliśmy rzetelny pakiet informacji o działaniach prewencyjnych, o działaniach operacyjnych. Opozycja grzmi, iż nic się nie dzieje w zakresie zapobiegania, że jest chaos, że samorządy, placówki medyczne w regionach działają bez jasnych wytycznych.

Panie Premierze! Tak, jest panika. Bo ludzie się boją. Bo wiedzą, że zrobiliście państwo z dykty i jak chłopaki z zapałkami podpalacie to państwo. Panie premierze, pan tyle mówi o tabelkach. Ile pieniędzy, skąd i dokładnie na co zamierzacie wydać? Bo tu słyszymy: 40 mln ze straży pożarnych, tutaj pan poseł Hoc opowiada o 100 mln. Panie premierze, konkrety. Ja bym chciała wierzyć jako obywatelka, jako matka i jako córka, że jesteście przygotowani na koronawirusa i że nie wykorzystujecie go do celów politycznych, ale patrzę na te puste ławy, patrzę na milczącego prezydenta, patrzę na brak zainteresowania i myślę sobie, że znowu robicie kampanię.

Panie Prezydencie! Wysoka Izbo! W walce z chorobami zakaźnymi bardzo ważna jest szybka i skuteczna diagnostyka. Dlatego chciałbym zapytać, czy państwo polskie dysponuje odpowiednią ilością testów do diagnostyki SARS-CoV-2. Nie ma pana posła. Pani poseł Elżbieta Płonka, klub Prawo i Sprawiedliwość.

Panie Prezydencie! Panie Premierze!

Panie Ministrze! Jak wiemy, Chiny to główny dostawca substancji czynnych do leków na europejski rynek, również na polski rynek.

Bardzo proszę.

Chyba byłby to najlepszy przekaz, jaki mógłby być.

Panie Prezydencie! Panie Marszałku! Panie Premierze! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! W sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa w Polsce konieczne jest, aby w zwalczanie rozprzestrzeniania się tej epidemii zaangażowały się służby podległe różnym ministerstwom. W związku z tym mam pytanie: Ile resortów, i które konkretnie resorty, jest zaangażowanych w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem, ze zwalczaniem epidemii zbliżającej się do Polski? Jak ta współpraca wygląda od strony logistycznej? Kto i za co konkretnie jest odpowiedzialny?

Panie Prezydencie! Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Chcę podkreślić, Wysoka Izbo, że zdrowie nie ma barwy politycznej, a zagrożenie zdrowia i życia zaczyna się od higieny. Pani poseł Katarzyna Sójka, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Prezydencie! Wysoka Izbo! Jako lekarz pracujący w szpitalu i przychodni jestem przekonana, że żadne procedury ani standardy postępowania w zakresie lecznictwa w Polsce absolutnie nie odbiegają od norm i standardów europejskich. Dlatego mam pytanie: Czy działania - i wprowadzone procedury działania - podjęte przez Ministerstwo Zdrowia odbiegają od działań podjętych w krajach Unii Europejskiej, czy też nie? Czy Ministerstwo Zdrowia konsultuje się i wymienia informacje z odpowiednimi resortami innych krajów Unii Europejskiej, czy nie? Jeszcze chciałam dokończyć pytanie.

Panie Prezydencie! Wysoka Izbo! Pytań było bardzo dużo. Zacznę od faktów, o których częściowo już mówiłem. Informacje o zachorowaniach we Włoszech. Zresztą komunikat Giuseppe Ippolito był jasny: dwie osoby są w dobrym stanie i nie ma groźby co do nowych ognisk wirusa. Dopiero dwudziestego drugiego zostały potwierdzone klastry, czyli ogniska zakażeń we Włoszech, a następnego dnia jako Polska zareagowaliśmy. Chciałem wyraźnie powiedzieć, że procedury zostały przekazane wszystkim jednostkom

To ogromna przykrość, że ta pani była tak potraktowana i miała taki stres związany z nieuzasadnionym podejrzeniem koronawirusa. Nieuzasadnionym, potwierdzam.

To była przestraszona, chora kobieta, która wymagała opieki i poczucia bezpieczeństwa.

Wystarczy decyzja powiatowego inspektora sanitarnego i te osoby otrzymają zasiłki chorobowe. Jednocześnie ustawa obecnie upoważnia nas do leczenia nieubezpieczonych z dotacji budżetowej. Było wiele pytań o bezpieczeństwo lekowe.

Jednocześnie dzięki SMoKL - znowu informatyzacja - wiemy, jakie są dostawy leków do Polski, jak one przebiegają.

Było pytanie któregoś z panów posłów o dobry poziom oddziałów zakaźnych, o to, które są dobre, naprawdę dobre albo tak bardzo naprawdę dobre, a które tak nie do końca naprawdę dobre. Z całym szacunkiem, nie wiem, co pan miał na myśli.